Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu sprawdzenia kworum. Bardzo proszę.

Dziękuję.

Stwierdzam kworum. Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 841. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 849. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, - o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 852, 850, 851 i 853. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Senat podjął uchwały w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, - o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uchwały Senatu to odpowiednio druki nr 854, 855 i 856. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych uchwał. Proponuję, na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu, rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwałach Senatu bez uprzedniego skierowania ich do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 845 i 852) Proszę pana posła Dariusza Bąka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoki Sejmie! W dniu 16 grudnia br. Senat na 19. posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i wprowadził do jej tekstu cztery poprawki. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w celu rozpatrzenia poprawek Senatu. Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich czterech poprawek. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Senat zgłosił do zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Głosujemy.

1 - za, przeciw - 449, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Nikt nie był za, przeciw - 448, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 847 i 850) Proszę panią poseł Agatę Wojtyszek o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 847. W dniu 17 grudnia 2020 r. komisje spotkały się i rozpatrzyły uchwałę Senatu z dnia 16 grudnia 2020 r., w której Senat zgłosił pięć poprawek.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 844 i 851) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedkładam sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, druk nr 851. Po rozpatrzeniu uchwały Senatu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia Komisja Finansów Publicznych rekomenduje odrzucenie wszystkich pięciu poprawek. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 846 i 853) Proszę panią poseł Mirosławę Stachowiak-Różecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, druk nr 846. Połączone Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły uchwałę na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy - Karta Nauczyciela. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W 2. poprawce Senat proponuje m.in., aby wyrazy użyte w art. 75 ust. 2a „prawa i dobro dziecka” zastąpić wyrazami „prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka” Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisje wnoszą o jej odrzucenie.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Prawo oświatowe Senat proponuje, aby wyrazy „w drodze umowy” zastąpić wyrazami „w drodze konkursu” Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 854) Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 20 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 20 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zechce nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 855) Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów uchwałę Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 848 i 849) Proszę pana posła Tadeusza Chrzana o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić sprawozdanie z posiedzenia odbytego w dniu dzisiejszym, na którym komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat do przedmiotowego projektu zaproponował sześć poprawek, w tym dwie o charakterze legislacyjnym: 1. i 6., które komisja rekomenduje głosować łącznie. Natomiast pozostałe cztery poprawki są poprawkami merytorycznymi. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek. Dziękuję. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o drogach publicznych. Łącznie z tą poprawką głosować będziemy nad poprawką 6. Głosujemy.

Głosowało 451 posłów. 1 - za, przeciw - 450, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Ogłaszam 10 minut przerwy.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy.

3 - za, przeciw - 444, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nikt nie był za, 448 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ogłaszam 5 minut przerwy i proszę Konwent Seniorów do

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 856) Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce nacisnąć

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Stwierdzam, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, że zachodzi przesłanka do reasumpcji głosowania. Wniosek o reasumpcję poddam pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do ponownego głosowania nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 841) Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionej propozycji? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 841, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Głosowało 449 posłów. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zanim wypowiem ostatnią formułkę, proszę państwa, mimo wszystkich trudności chciałabym wszystkim państwu życzyć spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. W związku z tym w dniu jutrzejszym obrady Sejmu nie odbędą się. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny kolejnego posiedzenia Sejmu zostanie paniom i panom posłom doręczony.